Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - o godz. 10.30. Bardzo dziękuję. Mam zgłoszenia wniosków formalnych. Bardzo proszę. 1 minuta, panie pośle. Szczęść Boże! Wysoka Izbo! Wnoszę regulaminowo o odroczenie rozpoczęcia tych obrad do czasu, aż pan marszałek będzie w stanie wraz z Prezydium ustalić, jaki jest właściwie porządek dnia, jaka materia ma być przedmiotem tych obrad, bo wybiła godz. 10, a na stronie Sejmu mamy informację tylko o tym, co na dobry początek. Potem, w południe, czyli już za niespełna 2 godziny, miałby się znowu zebrać Konwent Seniorów. Bardzo proszę, panie marszałku, narzućcie sobie jakieś ograniczenia w eskalowaniu niepowagi Wysokiej Izby. Podkreślam: koło Konfederacja nie uskarża się, tylko sygnalizuje, że to jest niepoważne. My jesteśmy w pełnym składzie - czy to w realu, czy to wirtualnie. Jesteśmy gotowi do pracy.

Pan poseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska, z wnioskiem formalnym. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów po to, by dzisiejsze posiedzenie Sejmu uzupełnić o punkt obejmujący informację prezesa Rady Ministrów o faktycznym stanie budżetu państwa.

Dzisiaj okazuje się, że król jest nagi. Panie Premierze! Natomiast pan powinien powiedzieć prawdę: Czy zmarnowaliście ostatnie 4 lata wzrostu gospodarczego i nie zreformowaliście finansów publicznych?

Dzisiaj, podczas tego posiedzenia Sejmu zmarnujemy kolejne godziny, tak cenne dla każdego Polaka i każdej Polki. Dzisiaj będziemy mówić o wyborach, dzisiaj będziemy słuchać pana premiera. Przecież możemy sobie włączyć Polskie Radio czy Telewizję Polską - tam już wszystko powiedziano: że pandemii właściwie już nie ma i że radzimy sobie lepiej niż wszystkie inne kraje na świecie.

Nie czas na gadaninę, nie czas na targi między panem prezesem Kaczyńskim a panem premierem Gowinem.

Dziękuję.

Informuję, że na podstawie art. 198a ust. 2 regulaminu Sejmu marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, podjęła decyzję o kontynuacji 9. posiedzenia Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Grupa posłów przedłożyła wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący informację prezesa Rady Ministrów nt. sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o tę informację. Proponuję, aby Sejm wysłuchał w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów nt. sytuacji.

Ale jeżeli. Ja wiem o tym, ale państwo zgodziliście się na 5-minutowe.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Informacja Prezesa Rady Ministrów nt. sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Bardzo proszę, panie premierze. Wysoka Izbo! Drodzy Rodacy!

Tak dzieje się we wszystkich polskich domach. Wiemy doskonale, że wszystko, co robimy, musi służyć ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Widzimy, w jaki sposób przyrasta liczba zachorowań w zachodniej Europie, widzimy, że te przyrosty są bardzo szybkie.

To powoduje, że bardzo wiele naszych działań w życiu publicznym, życiu społecznym, życiu gospodarczym musi dopasować się do epidemii. Musimy, walcząc z epidemią, jednocześnie starać się budować nowy model życia gospodarczego po to, żeby gospodarka ucierpiała jak najmniej. Jeśli nadal będziemy podchodzili z żelazną dyscypliną, z taką dyscypliną, z jaką do walki z koronawirusem podchodzi społeczeństwo polskie, jeśli nadal będziemy przestrzegali kwarantanny tak dobrze jak do tej pory albo może nawet lepiej, to - jestem o tym przekonany - będziemy w stanie poradzić sobie z pandemią koronawirusa o lepiej niż wiele innych krajów.

To wszystko powoduje, że musimy starać się ograniczać rozprzestrzenianie tej epidemii, jednocześnie starając się przywracać wiele form życia gospodarczego i funkcjonować w życiu publicznym w wielu obszarach, tak żeby ono zostało w możliwie mały sposób zakłócone. Bo ono zostaje zakłócone, to nie ulega wątpliwości. Funkcjonowanie ludzi na całym świecie zostało zakłócone i my w Polsce również funkcjonujemy w nowych, innych warunkach, w warunkach kryzysu epidemiologicznego. Myślę, że wszyscy to widzą, wszyscy to zauważyli. Szanowni Państwo! Wiele dyskusji publicznych dotyczy modeli zachorowań. My również słuchamy, analizujemy, słuchamy ekspertów i analizujemy bardzo wiele modeli, które mogą się zdarzyć. One są przede wszystkim naznaczone jedną charakterystyczną cechą, która zwykle jako mała gwiazdka jest gdzieś na początku każdej analizy - amerykańskiej, chińskiej, europejskiej czy polskiej. Otóż eksperci zdają sobie sprawę z tego, że to modelowanie jest obarczone ogromnym marginesem błędu.

Spodziewamy się, że szczyt zachorowań jest przed nami - nastąpi gdzieś w maju, w czerwcu. Jak mówi wielu ekspertów, promienie ultrafioletowe będą z całą pewnością pomocne w walce z koronawirusem, ale chcemy do tego czasu ograniczyć ilość zachorowań, a w szczególności wypłaszczać krzywą zachorowań. Amerykanie stwierdzają, że u nich być może szczyt zachorowań nastąpi w kwietniu. My nie wiemy, czy będzie to kwiecień czy maj, czy czerwiec.

Wśród tych problemów pierwszy, o którym powiem, to kwestia sprzętu. Sprzęt, dostępny sprzęt ochrony osobistej to bardzo ważny aspekt walki z koronawirusem. Dzisiaj mamy tego sprzętu cały czas jeszcze za mało, ale staramy się pozyskać go ze wszystkich kierunków świata (Dzwonek) i staramy się również odtworzyć produkcję krajową. W tym momencie warto z całą pewnością podkreślić, że jesteśmy przekonani, iż odtworzenie produkcji krajowej maseczek, fartuchów ochronnych, w przyszłości może też bardziej zaawansowanych sprzętów - pomoże, także w przyszłości, w walce z koronawirusem, jeżeli nie zaistnieje scenariusz bardzo optymistyczny, czyli szybkie wynalezienie szczepionki bądź szybkie zwalczenie tej pandemii. Gotowe są zapasy na kolejne tygodnie - 31 mln maseczek medycznych, rozdysponowano również 7 mln maseczek medycznych dla szpitali. Przede wszystkim pozyskujemy nowe ilości maseczek, fartuchów ochronnych, kombinezonów, gogli i respiratorów. Do Polski przyjechał transport 165 respiratorów z 1000 nowych zamówionych. Staramy się, jak widzicie, szanowni państwo, uprzedzać bieg wydarzeń. To dlatego właśnie tworzymy nowe miejsca na oddziałach zakaźnych, tworzymy nowe oddziały zakaźne, to dlatego utworzonych zostało 20 szpitali jednoimiennych. Przygotowujemy się również na dłuższą walkę z epidemią i dlatego musimy odbudowywać nasz polski potencjał produkcyjny. To już się dzieje. Kilkaset mniejszych i większych zakładów szwalniczych i nie tylko przestawiło swoją produkcję. To też jest pewnego rodzaju znak czasów, że w momencie kiedy nie wiemy dokładnie, kiedy będzie szczyt zachorowań, nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja jesienią, wiosną przyszłego roku, musimy na trwałe przebudować struktury produkcji w naszym kraju po to, żeby zapobiegać przyszłym ewentualnym nawrotom tej pandemii.

Już teraz do laboratoriów trafiło dodatkowe 150 tys. testów. Testy to też jest często temat debaty publicznej, więc teraz chcę parę minut poświęcić temu obszarowi.

Otóż z całą odpowiedzialnością chcę podkreślić, że te państwa, które miały taką liczbę zachorowań jak Polska obecnie, były na tym etapie, na jakim dzisiaj jest Polska, testowały o wiele mniej przypadków na 1 mln mieszkańców, i to niezależnie od tego, jaki to był kraj, czy Francja, czy Wielka Brytania, czy nawet Hiszpania i Włochy. Wystarczy sięgnąć do statystyk. A więc jeśli chodzi o liczbę wykrywanych przypadków na tym etapie rozwoju pandemii, o liczbę testów, które mamy zakontraktowane, to jest to 800 tys. testów, 800 tys. testów zakontraktowanych, 150 tys. dostępnych, 150 tys. testów już jest w drodze, w ciągu najbliższych paru dni będzie w Polsce, czyli mamy ogromny zapas testów.

Robimy wszystko, żeby nasza służba zdrowia była lepiej przygotowana w kwietniu, w maju, w czerwcu, w lipcu na dany etap walki z koronawirusem. Nikt na świecie nie wie, kiedy będzie szczyt, nikt na świecie nie wie, kiedy będzie spowolnienie, czy ono będzie gwałtowne, czy ono będzie o wydłużonym przebiegu krzywej.

Niepokój, jaki towarzyszy nam w ostatnich tygodniach, jest w pełni zrozumiały. On wynika z tego, że stoimy przed dużą, ogromną niewiadomą, niewiadomą zarówno w życiu społecznym, dla zdrowia publicznego, jak również w życiu gospodarczym. Kryzys, który jest udziałem państw całego świata, a w znacznym stopniu również państw zachodnich, państw najbogatszych, stał się przedmiotem ogromnej troski i analiz, ale zarazem z wielką pokorą najlepsi ekonomiści świata przyznają, że nikt takiego kryzysu się nie spodziewał. Dlatego tych wszystkich, którzy mówią: należy zastosować takie remedium, takie narzędzie, należy jeszcze trzy razy więcej opodatkować, znaleźć środki, żeby wydać je jak najszybciej, bardzo gorąco zachęcam do przeanalizowania tych wszystkich ekspertyz, którymi posługuje się rząd, którymi posługujemy się, żeby znaleźć najbardziej właściwą odpowiedź, bo trzeba podejść do tego z ogromną pokorą. Nikt nie wie, w jaki sposób będzie przebiegał ten kryzys, i trzeba dbać o siłę złotówki, o siłę i stabilność finansów publicznych państwa, o spójność polityki monetarnej, regulacyjnej, fiskalnej, finansowej w szerszym tego słowa znaczeniu, w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki narodowej. Pandemia do pewnego stopnia przypomina wpływ, jaki miały wszystkie kryzysy jednocześnie, ponieważ mamy do czynienia ze spadkiem cen surowców, z osłabieniem walut - dolar natomiast zyskuje na wartości, czyli jest to klasyczny przypadek osłabienia bardzo wielu walut świata, również euro do dolara, a więc nie tylko złotówka - oczywiście kryzys uderza kanałem majątkowym, następuje spadek cen różnych aktywów na całym świecie, ale także kryzys jest zupełnie nietypowy, ponieważ równocześnie uderza w stronę podażową i stronę popytową gospodarki narodowej, ba, wszystkich gospodarek na całym świecie.

Dlatego właśnie z dużą dozą ostrożności musimy podchodzić do wielu działań, które proponujemy. To chyba bardzo wiele mówi, podobnie jak analizy wszystkich najbardziej renomowanych instytucji ekonomicznych świata, które wskazują na to, że dzisiaj trzeba konsolidować swoje podejście w ramach polityk gospodarczych, trzeba z ogromną ostrożnością podchodzić do wielu działań związanych z jednej strony z dbaniem o gospodarkę, a z drugiej strony właśnie z podejściem do ograniczania koronawirusa, bo niestety kryzys zdrowotny coraz bardziej przepoczwarza się w kryzys gospodarczy we wszystkich krajach świata, co wyraźnie widać w bardzo bogatych krajach świata.

Tymczasem chcę Wysokiej Izbie zaraportować i drogich rodaków poinformować, że na dzień dzisiejszy 200 tys. firm w Polsce już złożyło wniosek do odpowiednich instytucji. Te wnioski już są rozpatrywane.

Na długiej liście składników tarczy antykryzysowej, które zaproponowaliśmy, znajdują się właściwie wszystkie instrumenty gospodarcze, finansowe, fiskalne, także monetarne, bo wejście ze wsparciem banku centralnego nie jest jakąkolwiek realną, konkretną pomocą finansową dla sektora bankowego. To robią Europejski Bank Centralny, amerykański bank centralny Fed, a także wszystkie inne banki centralne bogatych krajów zachodnich.

Polska mówi o tym głośno od kilku lat, od kiedy rządy sprawuje Prawo i Sprawiedliwość.

Przypomnę tylko, że to rząd Platformy Obywatelskiej w 2009 r. zrezygnował ze wspólnych zakupów, wspólnych zamówień. Wszyscy o tym wiedzą.

Do tej pory mieliśmy możliwość zastosowania coraz bardziej elastycznych źródeł czy coraz bardziej elastycznego zastosowania środków z funduszy strukturalnych, środków polityki spójności.

Przede wszystkim jednak, jak spojrzycie państwo na stenogramy z posiedzeń Rady Europejskiej, głos Polski jest jednoznaczny: potrzebujemy nowych środków w ramach Unii Europejskiej.

Polska jest gotowa uczestniczyć w mechanizmach gwarancyjnych w proporcjonalny sposób, żeby te mechanizmy gwarancyjne spowodowały możliwość emisji na rynkach światowych.

Wystarczy prześledzić stenogramy z posiedzeń Rady Europejskiej. Wszystkie kraje, również Włochy, Francja, także Hiszpania czy cała Grupa Wyszehradzka, upominały się o to, o co ja bardzo głośno się upominam, czyli o wspólną, solidarną politykę, której jest dzisiaj coraz więcej. Mam na myśli ten mechanizm elastyczności. Dobrze, że on jest, cieszymy się z niego, wskazywaliśmy na to, że on powinien być, i to się stało, ale muszą pojawić się nowe środki. 3 minuty temu powiedziałem, skąd te nowe środki mogą się pojawić: podatek cyfrowy, podatek od śladu węglowego, podatek od transakcji finansowych, podatek od jednolitego rynku, od wielkich międzynarodowych korporacji, a przede wszystkim likwidacja rajów podatkowych. Opowiedziałem Wysokiej Izbie również o tym, że Polska w aktywny sposób bierze udział w konstruowaniu nowych mechanizmów finansowania i montażu linii finansowo-kredytowych pod realizację różnych projektów infrastrukturalnych w zakresie służby zdrowia, ochrony zdrowia publicznego, które mogą być przydatne w przyszłości, ale ta przyszłość, tak jak powiedziałem na początku, jest bardzo niepewna. W związku z tym te mechanizmy, które udało się dzisiaj, na razie na papierze, wypracować, też są bardzo ważne i z tego też się bardzo cieszymy. Szanowni Państwo! Kończąc, chcę raz jeszcze podkreślić, że mierzymy się z sytuacją dramatyczną. Na świecie dzisiaj zarejestrowano 1250 tys. zachorowań, jest już kilka krajów, w których przekroczona jest liczba 100 tys. zachorowań, we Włoszech jest to powyżej 130 tys., w Hiszpanii również.

We Włoszech, w Hiszpanii te liczby są bardzo wysokie.

Dzięki temu wiemy, w jaki sposób budować szpitale polowe, gdzie najlepiej tworzyć nowe miejsca, czy one powinny być w wielkich halach, czy raczej w odosobnionych, mniejszych gabarytowo budynkach. To są doświadczenia, które zyskujemy. Dzieje się tak dlatego, że skutecznie, choć z pokorą, realizujemy jedną zasadniczą strategię: spowalniamy przyrost liczby zachorowań w porównaniu z tym, co dzieje się w Europie Zachodniej, w porównaniu z tym, co dzieje się w wielu innych krajach świata, również w Stanach Zjednoczonych.

Wszyscy o tym dzisiaj wiedzą. Musimy odszukać nowe punkty równowagi, nowe equilibrium po to, żeby rzeczywiście starać się żyć i pracować, a jednocześnie zapewniać najlepszą możliwą opiekę służby zdrowia wszystkim pacjentom, którzy zachorowali w Polsce, w tych okolicznościach rozwoju koronawirusa, w których się znajdziemy. A żeby tak się stało, to raz jeszcze zaapeluję o to, żeby zachować tę podstawową zasadę, co do której niemal wszyscy eksperci na całym świecie są zgodni: dystansowanie społeczne i zasady higieny, to co podkreślamy od kilku tygodni. Polacy w kwarantannie zachowują się bardzo odpowiedzialnie.

Nasze wspólne wysiłki, wysiłki wszystkich Polaków są niezbędne do tego, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i żeby móc wracać do tej nowej normalności, do tej normalności, za którą wszyscy tęsknimy. Jestem przekonany, że w naszych solidarnych wysiłkach doprowadzimy do tego, że będziemy potrafili przebudować nasze życie społeczne i gospodarcze w sposób odpowiedni do walki z koronawirusem. Bardzo dziękuję, panie premierze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 7-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pan poseł Tomasz Latos. Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Wszyscy ci ludzie codziennie bardzo ciężko pracują dla naszego bezpieczeństwa. Pamiętajmy w tym miejscu o pracownikach inspekcji sanitarnej. Często zbyt mało o nich się mówi. 16 tys. pracowników, którzy też są na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Oni, organizując pierwsze laboratoria, jako jedni z pierwszych podejmowali działania w tym zakresie. Podziękujmy służbom mundurowym, które dbają o to we wspaniały sposób.

Wreszcie to wielu pracowników, którzy nie mogli przerwać swojej działalności, którzy pracują chociażby w różnego rodzaju sklepach, dbają o to, aby dostawy były ciągłe, abyśmy byli zaopatrzeni w różnego rodzaju potrzebne na co dzień towary.

Pamiętam, jak nad tą ustawą pracowaliśmy. I pamiętam obawy, wówczas byliśmy w opozycji, czy te uprawnienia do wprowadzenia, czy w jednym województwie przez wojewodę, czy w całym kraju przez ministra zdrowia, z tymi wszystkimi obostrzeniami, z którymi spotykamy się na co dzień, nie mogą być jakimś polem do ewentualnych nadużyć, tym bardziej że przecież mamy stany wyjątkowe, w tym stan klęski żywiołowej, które można było wprowadzić zgodnie z istniejącą w Polsce konstytucją.

I takie zabezpieczenia zostały wprowadzone, i to zostały, szanowni państwo, wprowadzone jednomyślnie. Mimo zrozumiałych obaw opozycji ani jedna osoba się nie wstrzymała, wszyscy razem głosowaliśmy za tymi rozwiązaniami. Pamiętajmy, że warto i trzeba w niektórych sytuacjach pracować razem. Takim dobrym przykładem była chociażby specustawa dotycząca ochrony zdrowia, która nawiązywała do ustawy z roku 2008, kiedy potrafiliśmy wszyscy wspólnie pracować nad poprawkami. Też pamiętam, niektórzy z państwa brali udział w posiedzeniach komisji, kiedy potrafiliśmy razem dla dobra publicznego przyjąć poprawki - my jako strona rządząca wasze poprawki, a wy nasze poprawki, aby ustawę poprawić.

Patrząc obiektywnie na to, co dzieje się w innych krajach, na pewną nieodpowiedzialność niektórych rządów, nie będę wymieniał, w których państwach, można powiedzieć, że zareagowaliśmy bardzo wcześnie, a nawet w jakimś sensie nieproporcjonalnie wcześnie do sytuacji, kiedy jeszcze tej epidemii w Polsce nie było, bo przecież rząd, sztab kryzysowy działał jeszcze przed okresem pierwszych zachorowań w Polsce.

Podziękować należy, tak jak zresztą mówił pan premier, za działania społeczeństwa, za dyscyplinę, za dyscyplinę w kwarantannie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska pan poseł Borys Budka. Panie Marszałku! Puste słowa. Zamiast konkretnych propozycji niestety mamy kolejny festiwal ogólników. Tak, rzeczywiście pan może być ekspertem, jeśli chodzi o mówienie o ukrywaniu majątku i rajach podatkowych. Nie trzeba raju podatkowego, wystarczy przepisać majątek na żonę, prawda? Szanowni Państwo! Trzeba jasno, czytelnie powiedzieć: nie macie propozycji, a niestety nie skorzystaliście z dobrych propozycji polskiego Senatu, nie skorzystaliście z dobrych propozycji opozycji. Tutaj, w tym Sejmie, odrzuciliście każdą poprawkę. Gdzie byliście, kiedy proponowaliśmy, żeby każda firma, bez względu na to, ile zatrudnia osób, otrzymała pomoc od państwa? Głosowaliście przeciw. Gdzie byliście, kiedy proponowaliśmy 20 mld na służbę zdrowia? Głosowaliście przeciw. Gdzie byliście, kiedy upominaliśmy się o opiekunów osób niepełnosprawnych? Te dzieciaki nie mogą chodzić do szkoły, bo szkoły są zamknięte. Chcieliśmy objąć je pomocą. Jak głosowaliście? Przeciw. I dzisiaj mówicie o porozumieniu? Tak, jesteśmy do tego gotowi. Każdego dnia przychodzimy do Sejmu z propozycjami. Leżą ustawy senackie, leżą projekty Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej. Ale wy, zamiast rozmawiać o tych propozycjach, chcecie zmieniać Kodeks wyborczy. Przecież za 2 godziny, za godzinę będziecie proponować wprowadzanie głosowania korespondencyjnego - zamiast rozmawiać o propozycjach dla Polaków. W czasie pana wystąpienia otrzymałem kilkadziesiąt wiadomości. Płacząca matka trzylatka i jedenastolatka mówi o tym, że pracuje w hotelu. Nie może iść do pracy, bo zamknęliście je z dnia na dzień. Jakie są propozycje? Żadne. To jest tragedia ludzka, a wy śmiecie mówić o tym, jak ograniczać prawa obywatelskie, i będziecie proponować, żeby Poczta czytała nam korespondencję.

Komisja Europejska musi się upominać o prawdę. Porzućcie tę narrację. Bądźmy wreszcie razem, ale bądźmy na uczciwych zasadach. Polscy pracodawcy oczekują konkretnej pomocy. Polscy lekarze oczekują sprzętu ochronnego, oczekują godnego wynagrodzenia, oczekują tego, by zostać przetestowani.

No, na Boga! Bądźcie choć raz uczciwi! Uczciwość w czasach kryzysu to jest podstawowa wartość. Uczciwość wobec wyborców, ale też uczciwość wobec samych siebie. Apeluję o to, by zaprzestać tej propagandy.

Pan premier Morawiecki pouczał Niemców, mówiąc: bierzcie przykład z naszego budżetu. W Niemczech - 15 tys. euro dla każdego przedsiębiorcy. U nas zaproponowaliście 5 tys., i to pożyczki, którą trzeba oddać. Panie Premierze! Apeluję o uczciwość. Apeluję o to, by przeczytał pan te wypowiedzi internautów, które są po takim wystąpieniu. Jesteśmy gotowi, ale rozmawiajmy na poważnie. Testy, ochrona służby zdrowia, środki finansowe. I bądźmy solidarni w ramach Unii Europejskiej, bo tego oczekują od nas Polacy, wasi wyborcy, wyborcy Lewicy, PSL-u i nasi. Jesteśmy gotowi do tej pracy.

Panie Marszałku! Czy panu nie wstyd? Czy panu nie wstyd opowiadać tutaj o jakichś swoich wojnach, osobistych rozgrywkach z PSL-em, z Platformą Obywatelską, kiedy każdego dnia ludzie budzą się nie z troską, jak pan opowiada, ale z przerażeniem - dotyczącym pracy, dzieci, jedzenia, swojej przyszłości, swoich firm? My nie jesteśmy dzisiaj w stanie wojny politycznej, bo tego 38 mln ludzi nie chce. 38 mln ludzi dzisiaj prosi: niech rząd zajmie się rozwiązywaniem problemów. My jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi, i to jest nasza praca. Przedkładamy projekty, przynosimy gotowe rozwiązania. Mówimy: testujcie lekarzy raz na tydzień. A pan premier mówi, że chciałby, żeby były testy. Pan nie jest od chcenia, panie premierze. Pan jest od rozwiązywania problemów tu i teraz. Pan jest od tego, żeby zająć się tym, co mają zrobić dzisiaj ludzie, którzy z minuty na minutę tracą mieszkanie. To jest realny problem. To jest realny problem: co za chwileczkę samotne matki będą dawały dzieciom do jedzenia. To jest problem: w jaki sposób dzieci mają się dzisiaj uczyć. Chcemy móc zająć się tym, o czym mówi 38 mln Polek i Polaków: problemami i rozwiązaniami tych problemów. Ale do tego trzeba odwagi. Trzeba odwagi, panie premierze, żeby powiedzieć: Unia Europejska jest siłą, która może nam pomóc. Tylko musicie przestać ją obrażać i zacząć współpracować. Bo faktycznie przed nami jest wielki egzamin, przed nami jako społeczeństwem - z odpowiedzialności i solidarności. Przed wami - egzamin z rządzenia. Widzą to pracodawcy, przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, którzy muszą zwalniać ludzi, bo takie wprowadziliście dziury w swojej tarczy. Widzą to nauczyciele i nauczycielki. Widzą to osoby pozostające już teraz na bezrobociu przez wasze dziury w systemie. Widzi to medyk. Widzi to pielęgniarka, która worek na śmieci skleja taśmą klejącą i idzie do pracy na pierwszą linię frontu.

I jeżeli nie spojrzycie - nie na wielkie dane, panie premierze, jak ma pan to w zwyczaju, nie na tabele i nie na wyobrażenia excelowe - na normalnego człowieka, który ma codzienne problemy ze znalezieniem się i w tej trudnej sytuacji, i w tej izolacji, ale przede wszystkim z myśleniem co dalej, to oblejecie egzamin nie tylko z rządzenia (Dzwonek), ale i egzamin z patriotyzmu. My próbujemy wam na to nie pozwolić.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Pan premier mówił dzisiaj jak zwykle długo, ale niewiele. Te wszystkie prezentowane obietnice nie mają żadnego pokrycia w faktach. Wczoraj mieliśmy 475 nowych zachorowań i niestety kolejne 15 zgonów. W sumie ponad 4 tys. zakażonych. To są realne liczby. Dlaczego pan dzisiaj nie powie o konkretach? Dlaczego pan nie wspomniał, że w marcu prawie pół miliona osób straciło pracę? Dlaczego pan nie powiedział, że kilkaset tysięcy firm zawiesiło działalność albo po prostu zbankrutowało? Dlaczego pan nie mówił prawdy? Bo to przecież pana rząd szacuje, że za tydzień, w święta, będzie ponad 10 tys. zakażonych wirusem, to pana specjaliści z rządu, pana eksperci twierdzą, że w kwietniu straci pracę 3 mln osób. A wy czym się zajmujecie? Owszem, pracujecie, nawet po nocach pracujecie, ale na Nowogrodzkiej, gdzie od tygodnia trwają targi pomiędzy panem Kaczyńskim a panem premierem Gowinem. W jakiej sprawie? W sprawie wyborów. W ciągu tygodnia nie złożyliście nawet jednego projektu ustawy, ani jednego projektu, który mógłby w jasny sposób powiedzieć, jak będziecie pomagać pracownikom i przedsiębiorcom. Za to co zrobiliście? To pokazuje, jakie dzisiaj są wasze priorytety. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawiódł w godzinie próby, a pan osobiście bierze za to odpowiedzialność. Każdy dzień zwłoki to 100 tys. zwolnień pracowników. Pan to doskonale wie i ma pan to gdzieś. Dość tego. W społeczeństwie narasta bunt i najwyższa pora skończyć tę farsę z udawanym pomaganiem. Domagamy się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. To konstytucyjny sposób przeniesienia wyborów, szybki i skuteczny. Ma to też pełne uzasadnienie w stanie, w którym jesteśmy, w sytuacji epidemicznej. I niech nie przyjdzie wam do głowy wprowadzać stanu wyjątkowego, bo ludzie przyjdą po was szybciej, niż sobie myślicie. A jeżeli macie z tym problemy, nie macie własnych pomysłów, to skorzystajcie z naszych, z pomysłów Lewicy, które w tej Izbie złożyliśmy. Raz jeszcze panu przypomnę o tych pomysłach, chociaż tydzień temu z tej mównicy panu o tym mówiłem. Wtedy nie będziecie mieli problemów i będziecie robili to, czego oczekują Polacy. Po pierwsze, dofinansowanie przez państwo płacy na poziomie 75% dla każdego przedsiębiorcy, który utrzyma zatrudnienie. Po drugie, umorzenie na czas kryzysu kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Po trzecie, pokrycie przez państwo kosztów stałych dla firm: rachunków za gaz, najem, prąd, leasing na co najmniej 6 miesięcy. I po czwarte, wsparcie dla szpitali i podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. Każdy dotyczy obaw i strachu o przyszłość. To są te listy, panie premierze, to są te wszystkie listy. Co ma powiedzieć żonie mąż, którego firma właśnie się zamknęła? Co mają powiedzieć młodzi Janek i Marta ze Zgorzelca, którzy do tej pory pracowali na śmieciówkach, a mają zapłacić ratę kredytu? Nie słyszycie tego w PiS-ie, prawda? Nie słyszycie tej rozpaczy. Nie słyszycie lęku przed utratą pracy. Nie słyszycie, bo nie chcecie słyszeć. Ale dowiecie się. Zostawię te listy panu premierowi, żeby mógł pan odpowiedzieć milionom Polek i Polaków, jak zapłacić za prąd, gaz, leasing, kredyt. Pan się uśmiecha, panie premierze, ale chciałem panu powiedzieć, że dla wielu rodzin w Polsce. Kładę zatem przed panem premierem i przed Wysoką Izbą projekt dotyczący tego, jak uratować miliony ludzi, którym za chwilę zawali się świat. Robimy to jako Lewica, bo chcemy z panem i z pana rządem współpracować. Lewica proponuje zatem, żeby na czas kryzysu wprowadzić świadczenie kryzysowe dla każdego, kto w czasie epidemii stracił pracę albo zamknął firmę. Takie świadczenie w wysokości płacy minimalnej będzie wypłacane przez cały czas trwania kryzysu. Wierzę, że tym razem nie wyrzuci pan i pana rząd tych wszystkich poprawek do kosza, tak jak Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło 200 poprawek Lewicy w tamtym tygodniu. Odrzuciliście je, wiedząc, że to dobre poprawki i że pomogą ludziom godnie żyć. Na koniec, panie premierze, panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym przypomnieć, że od połowy stycznia pan premier Morawiecki i pan prezydent Duda zapewniali nas, że państwo jest gotowe na epidemię i kryzys. Dziś widać, że nas okłamaliście. Co gorsza, okłamaliście obywateli. Zmarnowaliście te 3 miesiące, a skala zaniechań jest olbrzymia. Lekarze i pielęgniarki coraz częściej chorują na koronawirusa, bo nie potrafiliśmy ich dobrze wyposażyć. Nic z tego. Zapowiadam, że Lewica będzie prowadzić białą księgę zaniedbań i nieprawidłowości w czasach zarazy. Spiszemy wszystkie wasze puste słowa i niespełnione obietnice. Odnotujemy każde miejsce, gdzie zawiedliście, i każdą śmierć, którą ukryliście. Nie odpuścimy wam, bo tego od nas oczekują Polki i Polacy. Niech pan zapamięta te słowa, panie premierze, bo Lewica będzie uważnie patrzyła panu na ręce. Dziś, właśnie dziś, 6 kwietnia, jest czas próby i odpowiada pan za każdą zmarnowaną godzinę, za którą historia wystawi panu rachunek. Lewica będzie stała w gotowości. Chcemy współpracować, bo Polska jest najważniejsza. Pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Słyszał pan przed chwilą głosy polityków, bardzo słuszne, które zwracają uwagę na sprawy najistotniejsze: życie i zdrowie, ochronę miejsc pracy, ratunek dla polskiej gospodarki. Te głosy pan może traktować, jak często nasze głosy, polityków, jako głosy w sporze.

Pani Dagmara pisze: Piszę do pana jako żona przedsiębiorcy, który ostatnie 19 lat swojego życia poświęcił budowaniu firmy. W tym czasie były chwile gorsze i lepsze, ale zawsze wychodziliśmy na prostą. Zbudowaliśmy biznes, który zatrudnia ponad 100 osób, prawie wszystkie na umowach o pracę. Inwestowaliśmy wszystkie zyski, bo wszyscy mówili, że tak trzeba. Teraz z dnia na dzień odcięto nas od wszystkich zamówień. Nie mamy nic. Na żadne wsparcie z tarczy nie możemy liczyć. Pracownikom, którzy są dla nas jak rodzina, musimy wręczać wypowiedzenia, i to tuż przed świętami. Serce pęka, jak widzę męża, który nie śpi, nie je, siedzi i się zamartwia, co jeszcze można zrobić. Nie wiem, co będzie dalej, ale wiem, że te wszystkie obietnice rządzących są nic niewarte. Pan Wiesław, rolnik z Teodozjowa w gminie Biała Rawska: Jako znany rolnik, społecznie aktywny, dostaję wiele informacji od rolników, którzy mają żal do rządu i ministra rolnictwa z PiS, że nie przedstawili propozycji pomocy dla sektora rolnego w obliczu zapaści gospodarczej wywołanej zakazami handlu w związku z walką z koronawirusem. Szczególnie dużo krytyki płynie ze strony rolników, którzy zajmują się produkcją i sprzedażą roślin. Dla wielu z nich okres wiosenny to żniwa, szczególnie dla producentów wczesnych warzyw i kwiatów jednorocznych, rabatowych. Wszyscy są w podobnej sytuacji, ponieważ bardzo poważnie ograniczono lub całkowicie zamknięto handel na zwykłych targowiskach i rynkach hurtowych. Skarżą się, ponieważ bardzo dużo zainwestowali w swoją produkcję - w drogie nawozy, infrastrukturę - a dzisiaj nie mają gdzie sprzedać wczesnych warzyw, botwinki, cebuli zimowej ze szczypiorkiem oraz kwiatów rabatowych. Jakby tego było mało, niektórzy zarejestrowani jako działy specjalne produkcji rolnej już zapłacili z góry podatek za cały rok 2020, ponieważ jednym ze sposobów określenia dochodów z tego źródła jest zastosowanie norm szacunkowych określonych w rozporządzeniu ministra finansów. Nikt z rządu nie przedstawił planu wsparcia dla rolników, których sytuacja jest dzisiaj bardzo ciężka. Pani Marzena, przedsiębiorca z Płocka: Jak zwykle zostałam pominięta w tej tarczy. Prowadziłam handel obwoźny i z dnia na dzień zostałam pozbawiona możliwości pracy, gdyż zostało zamknięte moje targowisko. Te pieniądze muszę przeznaczyć na moją składkę ZUS. Z czego mam zapłacić za wodę, prąd, ogrzewanie? A za co mam dać dziecku jeść? Bez pomocy nie przetrwamy. Niestety ostatnie wydarzenia związane z koronawirusem i odgórne zamknięcie sklepów w galeriach postawiło mnie i całą moją rodzinę przed widmem upadłości i straty dorobku całego życia. Z dnia na dzień zostałem pozbawiony możliwości jakiegokolwiek zarabiania pieniędzy, a to, że nasza firma jest firmą rodzinną, tworzymy ją z żoną i kilkoma pracownikami, postawiło nas w tragicznej sytuacji. Mamy problem z uzyskaniem kredytu obrotowego dla firmy i zaczynają nam się bardzo mocno piętrzyć płatności. Nasza firma w obecnym kształcie funkcjonuje od 5 lat i robimy coś, co kochamy. Niestety za chwilę może okazać się, że stracimy wszystko, wraz z domem i jakimkolwiek miejscem do zamieszkania. Niestety z dnia na dzień jesteśmy bez środków do życia. Panie premierze, to tylko niektóre z tych listów. Jeżeli one nie poruszą waszych serc, umysłów, waszej wrażliwości i będziecie wychodzić na tę mównicę i mienić się bohaterami. Prawdziwi bohaterowie są gdzie indziej. To są ci z listów, którzy walczą o każde miejsce pracy, to są ci w szpitalach, w sklepach, w których podają towary, i wszędzie tam, gdzie w trudnych warunkach pracują. To są prawdziwi bohaterowie i im należą się ukłony wdzięczności i wyrazy największego wsparcia, nie tylko słowami. Myślałem, że dzisiaj usłyszę od pana, panie premierze, i myślę, że wielu z tych, którzy piszą te listy, myślało, że usłyszą, jaka będzie i kiedy będzie prawdziwa pomoc. Co ze sprawami związanymi z działalnością handlową w kolejnych tygodniach?

Kiedy do tej pracy wrócą? Na te pytania nie usłyszeli odpowiedzi. I to jest propozycja dla pana, to jest wyciągnięta ręka. Po pierwsze, musimy utrzymać sprawność systemu ochrony zdrowia, zabezpieczyć, dać poczucie pełnego bezpieczeństwa wszystkim pracownikom ochrony zdrowia.

Chodzi też o stabilne wsparcie finansowe dla szpitali, których inne oddziały nie funkcjonują, i pokazanie ścieżki dostępu do ochrony zdrowia dla innych chorych, nie tylko dla tych, którzy są zakażeni koronawirusem. Po drugie, prawdziwa tarcza antykryzysowa z funduszem płatności Banku Gospodarstwa Krajowego, ze zwolnieniem z ZUS-u dla każdej firmy, z minimalnym wynagrodzeniem dla każdego pracownika, który ucierpiał z powodu koronawirusa. Po trzecie, pakt solidarności. Pakt solidarności na najbliższe miesiące pomiędzy opozycją a rządzącymi. Pakt solidarności, na podstawie którego nakreślimy na najbliższe 3, 4 miesiące czy 5 miesięcy działania, które powinien podjąć rząd, i nakreślimy te plany dla całego społeczeństwa.

Dziękuję bardzo. Teraz głos ma pan poseł Krzysztof Bosak, koło Konfederacji. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Obserwujemy zapaść państwa. Nie wszyscy to jeszcze widzą, ale za kilka tygodni zobaczą to nawet widzowie TVP. Dyrektor szpitala w Bytomiu zorganizował kwarantannę lekarzom na sali z chorymi na COVID, bez jedzenia i bez środków ochronnych. Dyrektor szpitala w Toruniu zakazał lekarzom zakładania maseczek ochronnych, bo przed niczym nie chronią, a poza tym sprowokują pozostały personel do zażądania ochrony.

Chodzą i dalej zarażają, mimo że chcieliby chronić nasze zdrowie. Takie rzeczy dzieją się w całej Polsce, ale wiemy o tym mało, bo lekarze mają zakaz wypowiadania się o tym, co dzieje się w szpitalach. Firmuje to wszystko minister Szumowski, który stał się najpopularniejszym politykiem w kraju, ponieważ wygląda, jakby był zmęczony - i pewnie jest bardzo zmęczony. A mamy dopiero sam początek epidemii. Gdziekolwiek spojrzymy, wybija się jakaś głupota, jakaś patologia w zarządzaniu, jakiś brak odpowiedzialności decydentów. Panie Premierze! Mści się obsadzanie wszystkich stanowisk z klucza politycznego i partyjnego. A jak wygląda przyjęte przez Sejm betonowe koło ratunkowe dla przedsiębiorców, które dla zmylenia przeciwnika zostało nazwane tarczą antykryzysową? Liczy 179 stron, a instrukcja obsługi - 172. Panie premierze, to jest biurokratyczny horror. Agencja Rezerw Materiałowych nie ma podstawowych wyrobów medycznych. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie ma pieniędzy dla zwalnianych pracowników. Nie będę już mówić, co stało się z Funduszem Rezerwy Demograficznej, który również nie mógł się uchować, a teraz i tak pewnie by się nie przydał. Cała nasza gospodarka nie jest w stanie do teraz wyprodukować wystarczającej liczby tak skomplikowanych i technologicznie zaawansowanych produktów jak maseczki, rękawiczki, nie mówiąc już o niezwykle trudnym do wyprodukowania płynie do odkażania. Tymczasem dla was od kilku dni najważniejszym tematem jest to, czy 10 maja odbędą się wybory. Im starczyło ostrożności, by przełożyć wybory, a wam nie. Gdy prezes Poczty Polskiej twierdził, że nie jest w stanie obsłużyć wyborów korespondencyjnych, został wyrzucony, a na jego miejsce powołaliście wiceministra obrony narodowej. A czemu za wszelką cenę dążycie do wyborów, panie pośle? Bo doskonale wiecie, jakie dramaty będą się odbywać przez kolejne miesiące. Uderzy w nas największa liczba zachorowań, całkowita zapaść szpitali, o które nie dbaliście przez lata, degrengolada gospodarcza, bezrobocie. Mordując gospodarkę i osłabiając ludzką odporność psychiczną, bardzo drogo kupujemy czas, do niczego go nie wykorzystując. Nie macie planu, żadnej przyjętej strategii, poza przeczekaniem. Nasze państwo ma w sobie jeszcze tyle siły i woli, by dać mandat fryzjerce samotnie wychowującej dzieci, która musiała pracować, by mieć na jedzenie. Pytanie, czy starczy tej siły, gdy ludzie masowo zaczną łamać zakazy mające wątpliwe podstawy prawne. A zaczną je łamać, bo już widać, że entuzjazm sprzed kilku tygodni wyparował. Frustracja będzie z każdym dniem rosnąć, w miarę kurczenia się oszczędności, których, jak wskazują dane makroekonomiczne, Polacy nie mają. Panie Premierze! Powiedział pan: koniec z rajami podatkowymi. Raje podatkowe to wielki ubytek dla budżetów państw. To jest najgorsza droga, jaką może pan przyjąć. To właśnie Polska powinna być rajem podatkowym dla Polaków. Zamiast domagać się od Brukseli trzech nowych podatków na nas nałożonych, niech pan wreszcie zacznie obniżać podatki w Polsce dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracowników. To jedyna rozsądna droga. Teraz głos zabierze pan poseł Grzegorz Braun. Szczęść Boże! Wysoka Izbo! Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Jaką agendę wy właściwie tutaj realizujecie? Każdy dzień, każdy tydzień ujawnia rozdźwięk między celami deklarowanymi a celami, które realnie osiągacie. Nie rezygnujecie z tego, nie odpuszczacie. Za parawanem, za zasłoną dymną pod pretekstem walki z wrażym wirusem budujecie już nie zręby, tylko wyższe piętra systemu totalnej inwigilacji, i to tak kuchennymi drzwiami, prawda? Nie przez ministerstwo bezpieki i nie przez ministerstwo obrony, tylko przez Ministerstwo Cyfryzacji - ono proponuje wszystkim Polakom taką aplikację: ściągnij sobie, Polaku, rodaku, obywatelu, na własnego smartfona takiego elektronicznego pastucha dla grzecznych obywateli. Co wy tu robicie? Czy wy sami wiecie, co to jest za agenda? A może starsi i mądrzejsi objawiają wam z dnia na dzień, co to jest za scenariusz, w którego odgrywanie tak bardzo się zaangażowaliście?

Nimi trzeba się opiekować - jasna sprawa. Ale zamykać kościoły? Zamykać lasy? Kto tam ma lądować w tej puszczy, że Polacy nie mogą wyjść na spacer, przewietrzyć się przy pięknym wiosennym słoneczku? To jest, jasna rzecz, obłęd. Polacy z dnia na dzień coraz lepiej to rozumieją. Obawiam się, że tak jak pan marszałek i pani marszałek, i całe Prezydium nie wie jeszcze, nad czym za parę godzin przyjdzie nam tu głosować - bo nie dowieźli taczkami tych ustaw, które w ostatniej chwili nam tu wrzucicie - tak popadam w coraz większą obawę, że i pan premier, i jego ekipa jadą tą kolejką, do której wsiedli, ale nie widzą celu. Padały z tej trybuny pytania, kiedy zaczniecie wychodzić z tego obłędu, jakim jest zamknięcie państwa, zamrożenie gospodarki.

Lista posłów zapisanych do głosu została zamknięta. Jako pierwszy pan poseł Tomasz Latos, klub Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Przyznam, że zabierając tu głos jako pierwszy, miałem nadzieję, że ta dyskusja będzie w wykonaniu każdego klubu koncyliacyjna i konstruktywna. Muszę powiedzieć, że nie w każdym przypadku tak niestety było. Mam wrażenie, że niektóre wystąpienia wręcz były jeszcze bardziej ostre. Szanowni Państwo! W tej sprawie, którą w tej chwili mamy, naprawdę musimy działać wspólnie. Naprawdę, tak jak w czasach najtrudniejszych, potrzebne są silne, mocne kierownictwo i wspólne działanie. Kończąc to, co teraz mówię, pytaniem, chciałem zapytać pana ministra zdrowia o dane, o których mówił tutaj pan premier, związane z kolejnymi zakupami, działaniami na rzecz wyposażenia w środki ochronne w naszym kraju.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nawet w tak poważnej sytuacji - a sam pan premier przyznał, że sytuacja jest dramatyczna - uprawiacie propagandę. Wszystko jest najlepiej robione przez nasze państwo. Tylko testów ciągle nie ma w takiej ilości, nie są tak dostępne, jak by oczekiwali lekarze. One gdzieś są, ale konkretnie ich nie ma. Ciągle słyszymy, że mają się znaleźć. Maseczki - słyszeliśmy, że maseczki sprzedano, kiedy było wiadomo, że zaczyna się kryzys w naszym kraju. Ciągle nie ma odpowiedzi na te pytania. Jak tutaj mówić o zaufaniu, o tym, że możemy coś razem robić, kiedy ciągle nie możemy sobie powiedzieć prawdy? Mówi pan, że testów mamy wystarczające ilości. Prezes Narodowego Banku Polskiego mówi, że mamy wielkie pokłady pieniędzy, a minister Gowin mówi o tym, że nie można wprowadzić stanu klęski żywiołowej, bo państwo tego finansowo nie wytrzyma. W jakim jesteśmy miejscu?

Pan poseł Ajchler?

Nowa normalność. Może od razu lepiej: nowa wspaniała normalność. Mam nadzieję, że pan, panie premierze, czuje te skojarzenia, które się siłą rzeczy nasuwają. Czy to jest już ten moment, w którym wszyscy będą zadowoleni: jedni kopiąc rowy, a drudzy je zasypując, panie premierze? Proszę się zdobyć na odrobinę szczerości wobec narodu, współobywateli, rodaków, i proszę poinformować, do czego to zmierza, w którą stronę nawiguje rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ogóle wie, w którą stronę nawiguje. Co się dzieje z tym, co w tle przecież nie umarło? Przecież starsi i mądrzejsi nie zapominają: 447, manewry Defender 2020, obrót bezgotówkowy - do tego wirus jest świetnym pretekstem.

Wysoka Izbo! Mamy Wielki Tydzień, dzisiaj jest Wielki Poniedziałek, jest tuż przed świętami. Wypada mówić w tym tygodniu prawdę. Naprawdę, to jest ten moment, kiedy nie powinniśmy kłamać. I mówię to do pana premiera: Nie powinien pan kłamać, w momencie kiedy nasze państwo jest w wielkim kryzysie, kiedy zamykacie ludzi w domach, kiedy zamykacie sklepy, parki, ulice i cmentarze. A jesteśmy nieprzygotowani, bo wy się tym po prostu nie chcieliście wcześniej zajmować. Cała pomoc, którą chce pan przekazać, ma iść przez banki. A ludzie pytają: Gdzie są te pieniądze? Dlaczego firmy nie mogą dostać tych pieniędzy, tylko dostaną je banki? Dlaczego ludzie mają płacić podatki w sytuacji, kiedy nie mają dochodów? To jest tragedia. Ludzie płaczą w domach, bo tracą prace, a wy się uśmiechacie. Postaramy się teraz połączyć z panią poseł Katarzyną Lubnauer, która jest w Sejmie w jednej z sal.

Niech pan siądzie, dobrze? Teraz nie ma pan.

Możemy wpuścić tyle osób, ile jest tu w tej chwili. Tak jest. Szanowni Państwo! Mamy sytuację, w której rząd, wiedząc, co się zapowiada, ponieważ od stycznia było o tym wiadomo, nie przygotował Polski ani Polaków do stanu epidemii. W związku z tym gra na czas. No dobrze, musimy się ratować. I gdyby nie wspaniała postawa Polaków, to wszystko by się nie udało. Ale mimo wszystko spójrzmy na statystyki. Oznacza to wzrost w ciągu 3 dni o 39%, prawie 40%.

Panie Premierze! Art. 233 konstytucji wyraźnie określa, iż ograniczanie podstawowych wolności obywatelskich czy gospodarczych i innych jest możliwe tylko w wyniku, w ramach wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - jednego z trzech stanów nadzwyczajnych. Tymczasem pana rząd od 2 marca wprowadza daleko idące ograniczenia wolności zwykłymi ustawami i rozporządzeniami. Czy prawdą jest, że tym samym wprost łamie pan konstytucję? Czy prawdą jest, że tym samym próbuje pan nie tylko utrzymać majową datę wyborów prezydenckich, ale także uniknąć obowiązku wypłaty odszkodowań, które obywatelom i obywatelkom gwarantuje konstytucyjny porządek prawny?

Dziękuję bardzo. Teraz proszę pana marszałka Zgorzelskiego, który zabierze głos zamiast pani poseł Ścigaj. Wysoka Izbo! 7 lutego podczas obrad senackiej Komisji Zdrowia - można skorzystać ze stenogramu - zarówno wiceminister zdrowia, jak i główny inspektor sanitarny zapewniali, że szpitale są przygotowane do walki z tym podstępnym wirusem. Zapewniali także, że to niegroźny wirus i że zalecenia WHO nie obejmują w grupie państw zagrożonych Polski. W tym samym czasie 7 lutego Agencja Rezerw Materiałowych pozbyła się 62 tys. masek pełnotwarzowych. Jak to świadczy o stanie przygotowania naszego państwa?

Nas wyklucza ze wspólnoty, mówiąc, że nie mamy nic wspólnego z Polską. Chciałbym, żeby pan zareagował.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Panie premierze, tyle pan mówił o tym, że Polska wyjątkowo dobrze radzi sobie z pandemią koronawirusa, że jest w stanie opanować zachorowania. Po prostu Polska mlekiem i miodem płynąca. Pytam więc, dlatego wciąż nie jesteście w stanie pochylić się nad problemami Polek i Polaków, dlaczego nie możecie zrozumieć, że ludzie codziennie dostają wypowiedzenia, a wasza tarcza jest zerowym rozwiązaniem przeciwko pandemii koronawirusa. Wasz szaleńczy plan utrzymania władzy za cenę zdrowia i życia Polek i Polaków jest chorym pomysłem.

Chcemy współpracować. Zacznijmy rozmawiać. Kiedy w końcu zdecydujecie się na oficjalne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej oraz realną pomoc przedsiębiorcom i pracownikom? Dziękuję bardzo. Mamy następną osobę, która zabierze głos. Bardzo proszę, pani poseł. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Lewica charakteryzuje się tym, że działa, zamiast tylko mówić. Podczas kiedy państwo w obozie Zjednoczonej Prawicy przepychacie się, kto jest ważniejszy: Jarosław Kaczyński czy Jarosław Gowin, my odbieramy każdego dnia dziesiątki, jeśli nie setki, telefonów od ludzi, którzy tracą środki do życia, bo tracą pracę. Tracą ją dlatego, że przez 15 lat rządów prawicy żaden rząd - ani Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ani Prawa i Sprawiedliwości - nie uporał się z problemem umów śmieciowych. Dziś z powodu śmieciowego zatrudnienia cierpią nie tylko pracownicy restauracji, nie tylko pracownicy gastronomii i turystyki, cierpią także ratownicy medyczni, czyli bohaterowie, którzy dziś każdego dnia narażają swoje życie i zdrowie. Jeżeli dziś zostaną objęci kwarantanną, nie są pewni, czy otrzymają wynagrodzenie. Dlaczego? Nie robicie tego także dzisiaj, w dniu kryzysu. W kolejnej wersji tzw. tarczy antykryzysowej nie znajdziemy niczego, co byłoby adresowane do osób zatrudnionych na umowach śmieciowych. Dlaczego nie interesuje.

Tak, więc jeszcze chwilę poczekamy. To pytanie już było zadane, panie pośle.

Dwie - z tego, co widzę. Okej. Rzeczywiście, są trzy, ma pan rację.

1 minuta, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Szkoda, że nie mogę panu zadać tego pytania wprost, ale chciałem zapytać o jedną rzecz. Kiedy pan premier zechce poinformować pana politycznego patrona i wodza ugrupowania rządzącego, pana Jarosława Kaczyńskiego, że ten kryzys to nie jest kryzys recesji, to jest egzystencjonalny kryzys całego państwa i narodu polskiego, że efektem tego może być nie tyle recesja, ile utrata 30 lat pracy pokolenia, całego pokolenia Polaków budujących niepodległą Polskę i gospodarkę w tej Polsce? Nie można dopuścić do sytuacji, w której to staje się przedmiotem gry politycznej.

Dziękuję bardzo, panie pośle.

Wysoka Izbo! Bezpieczeństwo wymaga odpowiedzialności. Bezpieczeństwo wymaga współpracy i staranności. Żeby Polacy mieli poczucie bezpieczeństwa i czuli się prawdziwie bezpiecznie, konieczne jest wprowadzenie paktu solidarności pomiędzy opozycją a rządem, pomiędzy rządem a opozycją - po to, żeby nakreślić plany działania na najbliższe miesiące, żeby Polacy wiedzieli, co się będzie działo za tydzień, za 2, za 3 tygodnie, kiedy nastąpi powrót do działalności gospodarczej, kiedy będzie powrót do szkoły, co z egzaminami na koniec podstawówki czy co z maturami. Nie wolno zostawiać tego na ostatnią chwilę. Ten pakt solidarności nakreślający warianty: bardziej optymistyczny, trudniejszy, taki, który jest najbardziej realny, rząd powinien przedstawić wspólnie z opozycją. Do paktu solidarności wzywam dzisiaj premiera Mateusza Morawieckiego, wzywam większość parlamentarną.

Szanowni Państwo! Panie Marszałku! Tymczasem słyszymy od pana premiera zapowiedź kolejnych trzech, nawet czterech podatków, które chce wprowadzić pan premier. Przecież to na końcu obciąży nas, konsumentów, i firmy, które w całym systemie nie tylko rynku polskiego, ale także rynku europejskiego funkcjonują. To jest po prostu nieprzyzwoite. Po drugie, jeszcze kilka miesięcy temu mówiliście państwo o tym, że cała Europa zazdrości nam wzrostu gospodarczego, tego wszystkiego, co jest domeną pracy milionów polskich firm. Tymczasem dzisiaj to właśnie polscy przedsiębiorcy zazdroszczą Europie systemu wsparcia. Jak to jest możliwe, że firma niemiecka może otrzymać po 3 dniach rejestracji 15 tys. euro, a firma powyżej 10 pracowników nie otrzyma praktycznie żadnej pomocy ze strony państwa?

Panie i Panowie Posłowie! To jest moment, kiedy ludzie zasługują na prawdę.

Polacy powinni to usłyszeć i powinni precyzyjnie wiedzieć, co robi rząd każdego dnia. I dlatego moje pytanie jest dokładnie o tryb działania rządu. Gdzie są sztaby antykryzysowe? Czy w tych sztabach są lekarze? Kto słucha dzisiaj lekarzy? W jakim trybie one podejmują decyzje? Co się dzieje z raportowaniem informacji na temat chorych i umierających? Jaki jest tryb podawania tych informacji? Kiedy Polacy stoją wobec takiej tragedii, jedyną odpowiedzią, jaką mogą usłyszeć, jest pełna prawda i precyzja. Dziękuję bardzo. Pan poseł Wiesław Szczepański, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Już niedługo mamy mieć egzaminy ósmoklasistów, a potem matury. Czy rząd nie zamierza jednak po prostu podjąć decyzji o tym, aby wydłużyć termin albo przenieść te egzaminy na późniejszy okres? Otóż, panie marszałku, w moim województwie - wielkopolskim, w mieście powiatowym w tej chwili zamknięty jest szpital, zamknięty posterunek Policji.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Jan Grabiec. Bardzo proszę.

Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Pytania, które dziś zadajemy, zadają sobie Polacy, którzy od 2 miesięcy obserwują to, jak epidemia pojawiła się najpierw w Europie, potem w Polsce. Zadają pytania o to, dlaczego nie ma dostępu do testów na koronawirusa, dlaczego osoby, które mają podejrzenia, że mogły zetknąć się z osobami zakażonymi, nie mogą się przebadać, dlaczego nie mogą być badani lekarze, pielęgniarki, pracownicy systemu ochrony zdrowia, ratownicy, dlaczego nie ma dla nich środków ochrony, nie ma maseczek, nie ma fartuchów, dlaczego nie daliście rady. Można by szukać odpowiedzi w waszych wypowiedziach sprzed 2 lat, w wypowiedzi ministra Szumowskiego, który 2 miesiące temu, kiedy był na nartach z prezydentem Andrzejem Dudą, powiedział, że cieszy się, że może odpocząć, bo w ministerstwie nie ma za dużo roboty.

Bardzo proszę, panie ministrze.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za troskę. Chciałbym przekazać, że pogłoski o moim skrajnym wyczerpaniu są przedwczesne i niesprawdzone. Jako żywo chyba musiałbym być wówczas skrajnie wyczerpany, gdybym coś takiego powiedział. Padały tutaj pytania o konkrety, poza wypowiedziami bardzo emocjonalnymi, w których właściwie nie postawiono konkretnych pytań.

Pytaliście państwo o testy. Mamy w tej chwili wykonanych ponad 85 tys. testów, tj. ponad 2200 na 1 mln mieszkańców i na 4 tys. zakażonych. Plasuje to nas w czołówce peletonu krajów, które były na tym etapie epidemii, powtarzam. Pytaliście państwo, jak testujemy. Oczywiście powtórzę po raz kolejny, bo być może nie oglądacie państwo mediów, być może nie słuchacie wypowiedzi w różnych stacjach, że medycy mają pierwszeństwo w testowaniu.

W ostatnich dniach poprosiłem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o to, żeby zaczął płacić za wszystkie testy we wszystkich szpitalach dla pacjentów i personelu, co jeszcze zwiększy potencjał testowania. Szanowni państwo, ja jako minister zdrowia nie zlecam testów, zlecają je lekarze, zlecają je inspektorzy sanitarni.

Oczywiście one gwałtownie będą się kurczyły, gdybyśmy nie przekazywali nowych testów, i oczywiście to robimy. Tak jak powiedział pan premier, mamy 800 tys. zakontraktowanych testów, 150 tys. jest rozdysponowanych do laboratoriów, 170 tys. jest na polskiej ziemi.

To mówimy, bo to jest fakt, z tym trudno dyskutować. Mówimy również, że mamy zakontraktowane 31 mln kolejnych maseczek, 28 mln maseczek hepa i 14 mln rękawiczek. To oznacza konkretne działania. I to nie oznacza, że jest fantastycznie, nie. To oznacza po prostu, że walczymy na rynkach całego świata o to, żeby te maseczki kupić.

Zostały wyasygnowane i wysłane maseczki i sprzęt ochrony osobistej do wojewodów. Wojewodowie będą te maseczki i ten sprzęt ochrony osobistej rozdysponowywać, również do DPS. To są dosyć konkretne informacje i konkretne liczby.

Wiemy, że walczymy o ten sprzęt ochrony osobistej na całym świecie. Na razie te transporty do Polski idą i będą szły, a my natychmiast, jak tylko będziemy je otrzymywali, będziemy je przekazywali dalej. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie informacji. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Zarządzam przerwę do godz. 12.20. Informuję, że wtedy odbędą się głosowania.

Wznawiam obrady.

Poproszę wszystkich państwa o naciśnięcie obojętnie którego przycisku dla stwierdzenia kworum. Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku.

Przypomnę, że stwierdzamy kworum, czyli naciskamy obojętnie jaki przycisk. Troszkę dłużej musimy poczekać, żeby sygnał doszedł do wszystkich państwa posłów.

Dziękuję bardzo i proszę o podanie wyników.

W obradach bierze udział 427 posłów, czyli stwierdzam kworum. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwanie posiedzenia. Przystępujemy do głosowania nad tym wnioskiem. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Informacja Prezesa Rady Ministrów nt. sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm przyjął informację do wiadomości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów nt. sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym przyjął informację do wiadomości. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiła opinię dotyczącą wniosku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 4, oraz zastosowanie klauzuli, o której mowa w art. 30 ust. 9 pkt 2 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Słyszę sprzeciw, panie pośle. Wniosek formalny.

Kto z pań i panów posłów jest za skróceniem terminów, o których mowa w art. 30 ust. 4 i ust. 9 pkt 2 regulaminu Sejmu, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął. Wysoka Izbo! Wniosek formalny. Wnoszę o zmianę sposobu przeprowadzania głosowania z niesprawnego na sprawny. Dostaję nieustannie informacje o problemach z połączeniem. Kiedy pani nie zajmowała tego miejsca zaszczytnego, pan marszałek Terlecki, jak odnotowałem, dwa lub trzy razy powiedział do mikrofonu, to powinno być w protokole: nie mamy połączenia. a więc są problemy techniczne, które czynią iluzoryczną tę wersję, że bierzemy udział w obradach plenarnych i że wszyscy mogą z równą sprawnością i zgodnością z własnym sumieniem oddawać tu głos. Oczywiście to nie był wniosek formalny, panie pośle. Proszę bardzo. Panie pośle, ten brak połączenia dotyczył wyłącznie połączenia wizualnego z posłami, którzy zabierali głos w dyskusji. Nie dotyczył on głosowania. Tak więc ten wniosek jest całkowicie nieuzasadniony. Dziękuję bardzo. Natomiast system głosowań to jest zupełnie inny system. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 316 i 317) Na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 2 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a także art. 30 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 w związku z art. 26 ust. 1 regulaminu Sejmu grupa posłów zgłosiła kandydaturę pana Bartłomieja Sochańskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Proszę panią poseł Annę Milczanowską o przedstawienie wymienionej kandydatury.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam kandydaturę pana mecenasa Bartłomieja Sochańskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Od blisko 40 lat jest adwokatem i radcą prawnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1987 r. wykonuje zawód adwokata, obecnie w kancelarii adwokatów i radców prawnych Sochański i Osiński w Szczecinie. Przez wiele lat był delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury. W stanie wojennym był obrońcą w procesach politycznych, doradcą podziemnych struktur związkowych. Po 1990 r. odbywał adwokackie staże zawodowe w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Danii. Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie europejskim, prawie karnym, prawie gospodarczym. Był jednym z pełnomocników rodzin katyńskich w sporze przeciw Federacji Rosyjskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W 2016 r. założyciel i prezes Szczecińskiego Towarzystwa Dialogu o Prawie, stowarzyszenia praktykujących prawników, adwokatów i radców prawnych mających na celu odbudowę społecznego zaufania do środowisk prawniczych.

Mecenas Sochański był ekspertem Rady Europy do spraw bezpieczeństwa w miastach. W 2004 r. został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi. W tym samym roku przyznano mu tytuł Mecenasa Kultury Szczecina. W 2006 r. został laureatem Bona Lex, nagrody „Gazety Prawnej” dla najlepszych prawników. W 2010 r. w 40. rocznicę wydarzeń grudnia 1970 otrzymał od ministra sprawiedliwości srebrny medal pamiątkowy. W 2015 r. został uhonorowany przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Krzyżem Zasługi na Wstędze. Zarówno wyróżniająca wiedza prawnicza, jak i bogate doświadczenie naukowe i zawodowe w dziedzinie prawa wskazują, iż pan Bartłomiej Sochański jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję, pani poseł. Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie opinii komisji.

Panie Premierze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą wniosku w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, druki nr 316 i 317. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 30 ust. 5 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 2 kwietnia 2020 r. powyższy wniosek do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu zaopiniowania. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu wymienionego wniosku na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2020 r. oraz przeprowadzeniu dyskusji postanowiła kandydaturę pana Bartłomieja Sochańskiego zaopiniować pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zgłosili się posłowie, którzy chcą zabrać głos w sprawie zgłoszonej kandydatury. Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Proszę bardzo o zabranie głosu panią poseł Kamilę Gasiuk-Pihowicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zmarłych liczymy dzisiaj w setkach, chorych liczymy dzisiaj w tysiącach. W tym samym czasie, kiedy cały świat walczy z epidemią koronawirusa, PiS zajmuje się obsadzaniem posad i stanowisk w instytucji, która kiedyś była Trybunałem Konstytucyjnym. Wysoka Izbo! Naprawdę chciałabym teraz zaapelować do posłów i posłanek PiS-u: nie marnujcie czasu. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni walczą teraz o zdrowie i o życie ludzi. Często nie mają rękawiczek, nie mają maseczek, nie mają testów, brakuje im respiratorów. Ludzie tracą miejsca pracy, źródła dochodu. Bankrutują firmy. A czym w tym czasie zajmują się posłowie PiS-u? Obsadzaniem kolejnych posad, stanowisk, poszerzaniem swojej władzy w cieniu epidemii, która jest jedną z najgorszych epidemii i przetacza się obecnie przez świat. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Przyjrzyjmy się w ogóle, kogo PiS chce wybrać do Trybunału Konstytucyjnego pod osłoną epidemii. Co wyróżnia pana Sochańskiego? Może wiedza prawnicza? Za to na pewno wyróżnia go legitymacja partyjna PiS, już od 2017 r. Zresztą rok później był kandydatem PiS-u na prezydenta Szczecina. Nawet teraz, w momencie głosowania, będzie członkiem PiS-u. I znów decydującym kryterium nie będzie wyróżniająca się wiedza prawnicza, ale będzie partyjna lojalność. A co skutecznie zwiększa partyjną lojalność? Co umacnia lojalność kandydatów PiS-u wobec partii? Oczywiście stanowiska w spółkach Skarbu Państwa i zarobione dzięki nim pieniądze. Otóż pan Sochański, jak dowiadujemy się z powszechnie dostępnych źródeł, jest m.in. członkiem rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Komu będzie wierny pan Sochański? Konstytucji? Czy może PiS-owi, partii, dzięki której zajmuje eksponowane stanowisko, lub zajmował eksponowane stanowisko, w jednej ze spółek Skarbu Państwa? Ile pan Sochański zarobił w spółkach Skarbu Państwa przez ostatnie 5 lat? Wysoka Izbo! To wszystko wskazuje na to, że PiS proponuje do Trybunału Konstytucyjnego kolejnego partyjnego żołnierza, a tym samym coraz bardziej zamienia trybunał w polityczne koszary dla emerytowanych działaczy PiS z różnych szczebli. My do tego ręki nie przyłożymy. Nie przyłożymy ręki do waszej walki o posady, stołki, o poszerzanie władzy w cieniu najgorszej epidemii na świecie. Proszę bardzo, pani poseł Anna Maria Żukowska, klub parlamentarny Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kandydatura pana mecenasa Bartłomieja Sochańskiego budzi nasze duże zastrzeżenia - z prostego powodu: on zajmuje miejsce, na które czekają pan sędzia Roman Hauser, Andrzej Jakubecki i Krzysztof Ślebzak. To są posłowie, którzy zostali legalnie wybrani. Teraz każda osoba, która zostanie wybrana, kiedy ci sędziowie czekają na powołanie przez pana prezydenta Andrzeja Dudę - tak na marginesie dodam, że Lewica złożyła projekt ustawy umożliwiający złożenie ślubowania tym sędziom przed marszałkiem Sejmu lub marszałkiem Senatu - będzie kolejnym sędzią dublerem, będzie delegitymizować po raz wtóry Trybunał Konstytucyjny, tak jak robią to pani Przyłębska, pani Pawłowicz czy pan Piotrowicz. Zajmujemy się wyborem do trybunału, który w tej chwili nie orzeka, dla którego naprawdę nie jest też dużym problemem, że jest jeden wakat. A tak naprawdę, tak jak powiedziałam, trzy osoby czekają. Zajmujemy się tym w czasie, kiedy jest epidemia, kiedy powinniśmy przyjmować takie ustawy, które pomogą ludziom, a nie partyjnym figurantom, którzy są nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości. Pan mecenas niestety nie odpowiedział na postawione przeze mnie pytanie, o kazus, który być może się wydarzy. On doskonale wie, że Prawo i Sprawiedliwość chce ominąć stan klęski żywiołowej i konieczność jego wprowadzenia. A jest taka konieczność z tego powodu, że umierają ludzie, że coraz więcej jest zarażonych, że w domach pomocy społecznej nie ma lekarzy, a pielęgniarki również są chore. Mam niestety duże wątpliwości co do bezstronności pana mecenasa, który, jak powiedziała moja przedmówczyni, jest połączony przez bardzo dużą siatkę powiązań finansowych ze spółkami Skarbu Państwa, jak też z samą partią rządzącą Prawo i Sprawiedliwość, której nadal jest członkiem. Dlatego klub parlamentarny Lewicy nie poprze tej kandydatury, tak jak nie poprze żadnej kandydatury, która będzie przedstawiana na miejsce wymienionych przeze mnie sędziów, którzy zostali legalnie wybrani i czekają na powołanie. Wysoka Izbo!

Zapraszam pana posła Grzegorza Brauna, Koło Poselskie Konfederacja.

Proszę bardzo, panie pośle. Siła wyższa, panie marszałku. Szczęść Boże raz jeszcze! No jakieś tam kadry macie przecież. Weterani Mumii Wolności - do Trybunału Konstytucyjnego. Dorosły człowiek, który wstąpił do tej formacji, musiał być obciążony deficytem - albo moralnym, albo intelektualnym. Współpraca z tą formacją, stanowiącą w swoim czasie przedłużenie tego centralnego ośrodka dezinformacyjnego i deprawującego Polaków, jakim była i pozostaje - już nie na tę skalę oczywiście - gazeta, gwiazda śmierci z ul. Czerskiej, formacja polityczna, która była tej formacji rozszerzeniem - to nie jest rodowód, który by kogokolwiek predestynował do tego, żeby być jednym ze stróżów prawa konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej. No i konsul Republiki Federalnej Niemiec?

Szanowni Państwo! Z powodu ostrożności procesowej umówmy się, że znajdziemy kogoś, kto nie przechodził procedur clearingowych żadnego obcego państwa. Do rzeczy, panie pośle. Do rzeczy. Czy pani marszałek będzie tutaj występować w charakterze stylistki dyktującej posłom, na jaki temat i w jaki sposób mają się wysławiać? Czy będzie takie oczekiwanie, żeby przedstawiać pani marszałek teksty wystąpień z tej trybuny do recenzji? Myślę, że tego nie ma w regulaminie, więc proszę też powściągnąć - dobrze? - swoją naturalną tendencję do bronienia partyjnych kolegów. Ale przede mną nie trzeba przecież nikogo bronić, ja się do gardła nie rzucam. A więc sięgnijcie do tych waszych kadr partyjnych i znajdźcie kogoś, kto nie cieszył się ani zaufaniem Bronisława Geremka czy Adama Michnika, ani zaufaniem rządu Republiki Federalnej Niemiec. Tylko bardzo proszę, żeby to znowu nie był ktoś, kto w innych aspektach będzie wyczerpywał, jak by to powiedzieć, znamiona realności konstrukcji ustrojowej, którą przed laty określiłem jako kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym, co rzecz jasna w tej kadencji trzeba rozszerzyć i powiedzieć: żydowsko-amerykańskim zarządem powierniczym. Znajdźcie jakiegoś kandydata, przedstawcie go w normalnym trybie, dajcie sobie czas na to i wtedy zastanowimy się, czy tej kandydatury nie popierać. Tymczasem nie możemy. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Nikt o zdrowych zmysłach nie ma wątpliwości, że dzisiaj nie powinniśmy zajmować się wyborem kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, instytucji, która w istocie od dawna już straciła przymiot kolejnego elementu w systemie konstytucyjnym, bowiem poprzez swoją pauperyzację instytucjonalną utraciła zdolność wykonywania funkcji konstytucyjnych. Spadek zaufania społecznego mierzy się ilością obywatelskich skarg składanych do Trybunału Konstytucyjnego, trybunału, który był atakowany, że w 2015 r. wydał tylko 173 orzeczenia. Tymczasem w 2018 r. wydał już tylko 72. Wtedy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nazywani byli przez polityków obecnej partii rządzącej leniami, a posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego określano jako spotkania przy ciasteczkach i kawie. Jak dzisiaj można zdefiniować coś, co niesłusznie jeszcze czasami nazywane jest Trybunałem Konstytucyjnym, jeżeli do panteonu gwiazd dołączyli państwo Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowski?

Dzisiaj, szanowni państwo, tak jak powiedziałem na początku, nie powinniśmy zajmować się tymi sprawami, ponieważ codziennie setki firm bankrutują, codziennie tysiące naszych rodaków tracą miejsca pracy. Zamiast każdą minutę tej debaty poświęcić na to, żebyśmy mogli stworzyć system pomocy i tę dziurawą tarczę wypełniać treścią merytoryczną, dzisiaj stajemy w Wysokiej Izbie po to, aby dyskutować nad kolejną kandydaturą na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, która oczywiście większość parlamentarną zyska i kandydat zostanie wybrany. Tylko czy jeszcze, tak jak powiedziałem na początku, osoby zasiadające tam mogą posiadać przymiot sędziego i czy w ogóle ta instytucja jeszcze jest godna nosić nazwę Trybunału Konstytucyjnego?

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po pierwsze, należy powiedzieć kilka słów na temat tej niebywałej po prostu demagogii, z jaką mieliśmy tutaj do czynienia. Te wszystkie opowieści, że zajmujący pół godziny czy godzinę wybór przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, ale przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w tym samym znaczeniu, w jakim przedstawicielami innych partii, a w szczególności Platformy Obywatelskiej, byli wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego poprzednich kadencji. Na tym polega właśnie ta demagogia, bo z jednej strony nie ma tutaj mowy o żadnej stracie czasu, bo ta strata czasu to jest po prostu fikcja. W tej chwili nie ma żadnej możliwości podjęcia pracy nad innymi sprawami, a te, które będą, zostaną jeszcze dzisiaj wykorzystane. Po drugie, skład obecnego Trybunału Konstytucyjnego jest, po pierwsze, całkowicie legalny.

Ten wybór od samego początku był całkowicie bezprawny, był bez prawnego znaczenia. I chciałbym, żeby państwo o tym pamiętali. To wszystko, co uczyniliśmy później, było całkowicie zgodne z prawem. A decyzja Trybunału Konstytucyjnego podjęta bez przestrzegania jakiejkolwiek procedury była decyzją o wartości świstka papieru. Po prostu żadna tego rodzaju decyzja poza procedurą nie ma żadnego prawnego znaczenia. I chciałbym, żeby to w końcu zostało bardzo wyraźnie powiedziane, bo nieustanne powtarzanie o jakichś sędziach dublerach to jest po prostu nadużycie, ciężkie nadużycie, to jest oszukiwanie opinii publicznej. I jeszcze raz wracam do tej pierwszej sprawy. Wybieraliście posłów, wybieraliście działaczy Platformy Obywatelskiej czy przedtem Unii Demokratycznej - a tak się zdarza, że niektórych z nich nawet osobiście znałem, nawet razem działaliśmy w podziemnym Komitecie Helsińskim, ale byli wyraźnie po waszej stronie - i to było w porządku. Teraz wam się nie podoba, bo trybunał, który w gruncie rzeczy jest bardzo pluralistyczny (Dzwonek), nie jest taki, jak wy chcecie. Przechodzimy do głosowania. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę pana Bartłomieja Sochańskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 regulaminu Sejmu Sejm wybiera sędziego Trybunału Konstytucyjnego bezwzględną większością głosów. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem pana Bartłomieja Sochańskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm wybrał większością głosów pana Bartłomieja Sochańskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziś obradujemy nad ważnymi rzeczami dla Polaków, ale na pewno do tych rzeczy nie zalicza się powołanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na to poświęciliście państwo wiele minut, a w momencie, kiedy był czas na zadawanie pytań przez parlamentarzystów, wasz system zawiódł. Dlatego, korzystając z okazji, że pani marszałek dopuściła mnie jednak do głosu, chciałbym zapytać pana premiera, czy ma świadomość, że w moim rodzinnym mieście, w Radomiu, w jednym szpitalu już w tej chwili chorych jest 184 pacjentów, w tym 102 medyków. Panie Premierze! W jaki sposób udzieli pan pomocy mojemu miastu? Co pan zaoferuje dla Radomia, dla Grójca i dla Nowego Miasta nad Pilicą? Również pytanie bardzo ważne, zasadnicze: Czy miał pan i czy ma pan świadomość, że dziś najważniejsze jest badanie medyków? Bo to medycy, źle wynagradzani medycy pracujący na kilka etatów, którzy muszą zarabiać na swoje rodziny, dziś rozsiewają koronawirusa. W związku z tym zwracam się do pani z wnioskiem formalnym o zmianę sposobu procedowania w porządku obrad. Ten wniosek był już zgłaszany, w związku z tym nie będę poddawała go znów pod głosowanie. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., druki nr 314 i 314-A. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu. Jest to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przyjęcie propozycji uzupełnienia porządku dziennego oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., druki nr 314 i 314-A, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Wniosek nie uzyskał większości.